Zdrowia - godz. 17, - do Spraw Kontroli Państwowej - godz. 18, - Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki wspólnie z Komisją Zdrowia - godz. 19.30.

Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! W imieniu Komisji Zdrowia mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskich projektach ustaw.

Na posiedzeniu komisji przyjęto bez sprzeciwów jako druk wiodący druk nr 683, rozpatrując wszystkie te dokumenty razem i uwzględniając stosowne zapisy z pozostałych druków w trakcie procedowania tego druku wiodącego.

Chcę podkreślić dobrą pracę, którą przez wiele godzin wykonano w Komisji Zdrowia, którą mimo różnych stanowisk, także i sporów, udało się sprawnie i merytorycznie przeprowadzić.

Pacjenci, obywatele czekają na tę ustawę, która reguluje szereg ważnych kwestii zdrowotnych, a także organizacyjnych i innych. Mam nadzieję, że polski Senat równie szybko i bez zbędnej zwłoki zajmie się procedowaniem nad tą ustawą. Jestem przekonany, że jest to coś, na co czekają wszyscy w Polsce. Dziękuję, panie pośle, za przedstawienie sprawozdania, ale też za tę ciężką nocną pracę. 6-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Otwieram dyskusję. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Bolesław Piecha. Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość chciałbym przedstawić stanowisko wobec wyniku prac komisji, urobku komisji dotyczącego projektów ustaw zawartych odpowiednio w drukach nr 684, 685, 686 klubów opozycyjnych oraz wobec projektu ustawy zaproponowanego przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość zawartego w druku nr 683. Wybrano, tak jak powiedział przewodniczący, druk wiodący, czyli najbardziej obszerny projekt, propozycję ustawową dla Wysokiej Izby, niemniej muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony ze współpracy. Dyskusja była długa, bo praca była żmudna, materia bardzo skomplikowana, dotycząca wielu aspektów naszego życia.

Z czego jestem bardzo zadowolony? Może najpierw powiem o tych trudniejszych sprawach. Z tego, że wreszcie zostanie uregulowana sprawa obowiązku noszenia maseczek, masek, przyłbic itd. Wiemy dziś z różnych doniesień prasowych, różnych doniesień, pism fachowych i od ekspertów, że na dzisiaj jedynym sposobem zapobiegania szerzenia się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 jest po prostu noszenie maseczki, dystans społeczny i dezynfekcja. Nie mamy innego sposobu i w dającej się przewidzieć przyszłości - a pracujemy jednak w czasach bardzo gwałtownych zmian - nie spodziewamy się, żeby doszło do jakiegoś ogromnego przełomu w tym roku. Dzisiaj będzie to już obowiązek wyrażony w ustawie, a nie jak dotychczas w rozporządzeniu. W związku z tym opinia prawna w sprawach przed sądami - bo one się toczyły - będzie jednoznaczna. Powiem więcej, przyjęliśmy również poprawkę Lewicy i pani poseł niezależnej, żeby sprzedawca mógł odmówić sprzedaży towaru, jeżeli ktoś w sklepie nie zakrywa nosa i twarzy. Znamy tę słynną sprawę, co prawda pojedynczą, ale takie kazusy są i chcieliśmy to uregulować. Oczywiście są jeszcze pewne trudne sprawy dotyczące głównie rozliczeń. W dalszym ciągu jest pewna pula środków finansowych, która do tych przedsiębiorców jest kierowana, i każdy się może o nie ubiegać, ale - mówiąc kolokwialnie - będzie się musiał wyspowiadać, czy poprzednie środki wydał zgodnie z przeznaczeniem. To nie jest tak, że przedsiębiorca będzie musiał przedstawiać jakieś skomplikowane raporty, wielostronicowe sprawozdania, ale będzie musiał napisać proste oświadczenie, że środki, które zostały przekazane w ramach tarczy, wykorzystał zgodnie z przeznaczeniem. Z czego jestem zadowolony? Zadowolony jestem przede wszystkim z tych wszystkich spraw, które służą pacjentom. A pacjentom służą te sprawy, które wiążą się z możliwością usprawnienia opieki nad nimi. Otóż przede wszystkim poszerzyliśmy, o ile to było możliwe, możliwość szybkiego przeszkolenia fachowych pracowników ochrony zdrowia w pobieraniu wymazu. To ważne. To nie jest tak, że testujemy, bo wynik będzie dobry, tylko trzeba ten wymaz, to badanie przeprowadzić profesjonalnie. W związku z tym skorzystamy z różnych pracowników ochrony zdrowia w oparciu o Państwowe Ratownictwo Medyczne, również o służby ratownicze wojskowe, żeby po prostu powiększyć pulę ludzi, którzy fachowo pobierają wymazy. Druga sprawa dotyczy już pracowników, którzy są na pierwszej linii frontu, i to nie tylko pracownicy szeroko rozumianej ochrony zdrowia - to są również pracownicy służb: Policji, wojska, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to są również pracownicy straży pożarnych, to są pracownicy samorządowi, tacy jak strażnicy gminni. I zaproponowaliśmy im, że w przypadku, kiedy z powodu czynności podejmowanych z zakażonym koronawirusem dojdzie do zarażenia, a tym samym w konsekwencji albo leczenia, albo kwarantanny, albo izolacji, będą pobierać zasiłek w wysokości 100% należnego świadczenia ZUS-u, a nie, jak dotychczas przewiduje ustawa, 80%. Tę grupę poszerzyliśmy o pracowników Służby Więziennej, bo w więzieniach też są szpitale, musimy to, może z bólem, chciałbym, żeby było inaczej, uznać, i pracowników opieki społecznej, którzy pracują w noclegowniach, w domach dla bezdomnych, oni też mogą z tego skorzystać. Tak, proszę państwa, nie będziemy karać lekarzy, zwłaszcza tych lekarzy, którzy nie są specjalistami, za niezawinione błędy lekarskie. To się w każdej działalności medycznej zdarza i byłoby wyjątkową niesprawiedliwością, żeby traktować ich bardzo surowo. Jak zapowiedziałem wczoraj, jak zapowiedział premier Morawiecki, to wynagrodzenie wzrośnie o 100%, czyli będzie to 200% dzisiejszej pensji. Było ciężko, ale daliśmy radę. Na koniec w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość chciałem na ręce pani marszałek złożyć wniosek o niezwłoczne przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 bez odsyłania do komisji poprawek i wniosków zgłoszonych do tego projektu ustawy, oczywiście po doręczeniu ich posłom. Uzasadniam to tym, że jest bardzo dużo zgłoszonych wniosków mniejszości, nad którymi i tak bez rozpatrzenia przez komisję będziemy głosować. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Każdy projekt ustawy, który dotyczy walki z pandemią, powinien wpisywać się w strategię rządu, w strategię przemyślaną, spójną, która jest obudowana dobrymi przepisami, dobrym prawem, dobrymi ustawami. Dobrym prawem, które powinno chronić życie i zdrowie obywateli, ale także chronić wszystkich tych, którzy na pierwszej linii frontu walczą o nasze bezpieczeństwo, walczą o nasze życie i zdrowie. Niestety jest inaczej. Rząd strategii nie przemyślał, nie był też konsekwentny, nie komunikował się z obywatelami.

Odrzucił też ponad 120 poprawek, które przyszły z Senatu. Padło też wiele nieodpowiedzialnych słów premiera i przedstawicieli rządu, bo wirus nie jest w odwrocie i nie jest tak, że nie ma się czego bać. Tak mówił, jeszcze nie tak dawno, w lipcu, pan premier Morawiecki. Bo nie byliśmy przygotowani na każdy rodzaj epidemii - tak twierdził pan minister Dworczyk. Dziś zbieramy żniwo tych bardzo nieodpowiedzialnych słów i działań rządu. Tego nie da się niestety nadrobić, bo każdy dzień przynosi tragiczne statystyki wykrytych zakażeń, zgonów, zajętych respiratorów, zajętych łóżek. Słyszymy tragiczne rozmowy ratowników medycznych z dyspozytorami. Wszyscy to widzimy i coraz bardziej się boimy. Boimy się, bo widzimy, jak w chaosie pogrąża się służba zdrowia, a premier zamiast z pandemią walczy z prawdą. A prawda jest taka, że doszliśmy już do ściany. Według premiera jest świetnie, bo jak mówi, łóżek, respiratorów, personelu medycznego mamy ponad miarę. Mamy też dostęp do szczepionek przeciwko grypie, a gospodarka ma się świetnie. Przestajemy być takim liderem, o czym mówi pan premier Morawiecki, kiedy wyłączy się telewizję publiczną i wyjdzie do ludzi - zajrzy do szpitala, porozmawia z ratownikami medycznymi, zajrzy do sanepidu, który jest obciążony pracą, i porozmawia z nauczycielami, którzy też coraz bardziej się boją. Trzeba skończyć z propagandą sukcesu, bo nie można w nieskończoność udawać, że wszystko jest okej. Wczoraj dzięki temu, że we wtorek do pracy nie przyszło 28 posłów Zjednoczonej Prawicy, mogliśmy bez chaosu pochylić się nad kolejną rządową wrzutką przyjętą przez posłów. Dzięki temu projekt nie przejechał się ekspresem w pracach legislacyjnych w Sejmie, bez konsultacji i w chaosie. Mogliśmy skupić się na tym, żeby porozmawiać ze środowiskiem medycznym, samorządowcami, z dyrektorami szpitali, z ratownikami medycznymi, porozmawiać o szczegółach tej ustawy i przygotować dobre poprawki - dobre poprawki dla obywateli, dobre poprawki dla tych, którzy ratują nasze zdrowie i życie. Na posiedzeniu Komisji Zdrowia, które trwało wczoraj od godz. 14 do prawie godz. 2 w nocy, przez 12 godzin pracowaliśmy merytorycznie nad wszystkimi poprawkami, które zgłaszaliśmy. Niestety tylko cztery poprawki zostały przyjęte.

Strażnicy miejscy, ci, którzy są delegowani do walki z COVID, będą objęci takimi samym przepisami jak inne służby. Niestety kilkadziesiąt innych ważnych poprawek, które znacząco wpłynęłyby na poprawę pracy służby zdrowia i w ogóle na funkcjonowanie służby zdrowia w tym trudnym czasie, zostało odrzuconych. Niestety została odrzucona poprawka, która dotyczyła zwiększenia funduszu celowego o 5 mld, a tym samym niestety rządzący zrezygnowali z zakupu 10 mln szczepionek przeciwko grypie i co najmniej 100 tys. testów dziennie, bo na to byłyby te pieniądze. Niestety nie przeszła poprawka, która dawała ustawową gwarancję 200% wynagrodzenia dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia, którzy walczą z COVID, a nie tylko dla tych, którzy są delegowani przez wojewodów. Niestety nie przeszła poprawka, która mówiła o likwidacji możliwości odwołania dyrektora szpitala decyzją ministra zdrowia. Nie przywrócimy też handlu w niedziele. Nie przeszła również poprawka, która przeznacza na finansowanie ochrony zdrowia od 2021 r. corocznie środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6% PKB. Nie przeszła również poprawka, która dotyczyła zmian w dodatkowych zasiłkach opiekuńczych dla dorosłego opiekującego się dzieckiem z powodu COVID.

Drodzy Państwo! Liczymy na to, że w drugim czytaniu - bo będziemy składać ważne poprawki - jednak rządzący przychylą się do nich, ponieważ one dotyczą nas wszystkich. One dotyczą życia, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. Pamiętajmy też, że procedowanie nie kończy się w Sejmie. Liczymy również na Senat, który pochyli się także merytorycznie nad tym projektem ustawy, tak żeby ten projekt [[Dzwonek]] był kompletny i spełniał wszelkie oczekiwania obywateli, ale także tych, którzy walczą o nasze życie i zdrowie. Dziękuję, pani poseł. W imieniu klubu parlamentarnego Lewica głos zabierze pani poseł Magdalena Biejat. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Pan premier mówił wczoraj o drodze środka. Jeśli mam być szczera, to mnie nie interesuje w tej chwili, czy idziemy pośrodku, na przełaj, czy dookoła. Myślę, że Polaków też to nie interesuje. To, co nas interesuje, to dokąd ta droga prowadzi, jak długo będziemy nią iść i czego się mamy spodziewać. Na tym polega strategiczne myślenie i tego dzisiaj oczekują Polki i Polacy. Szkoda tylko, że niewiele z niej wynikło. Lewica pytała, jaki scenariusz przewidujecie na wypadek, gdy zabraknie respiratorów, jak chcecie działać, gdy dzienna liczba zachorowań będzie wynosiła 10, 20, 50 tys. Jaki macie plan B? Nie poznaliśmy odpowiedzi na te pytania ani w zeszłym tygodniu, ani w tym. Premier powiedział wczoraj, że wzrost zakażeń wynika z większej mobilności społecznej od września. Mówił o młodzieży, która jest pasem transmisyjnym epidemii. No cóż, nie trzeba geniuszu, aby te dwa fakty połączyć. Jeśli otwieracie szkoły w normalnym trybie i nie wprowadzacie nawet tak minimalnych środków zapobiegawczych jak obowiązek noszenia maseczek, nie zmniejszacie zagęszczenia w przeludnionych szkołach, to czego się spodziewacie? Alarmowaliśmy i wypytywaliśmy o to całe wakacje. Tydzień temu apelowaliśmy: zarządźcie przynajmniej 2 tygodnie przerwy w nauce, tylko 2 tygodnie. W tym czasie przebadacie uczniów i pracowników, zbierzecie rzetelne dane o tym, jak koronawirus rozprzestrzenia się w szkołach. Ten czas pozwoli na spowolnienie rozwoju epidemii, a potem uruchomcie szkoły w systemie rotacyjnym, tak by liczba uczniów pozwalała na dystansowanie. Zamiast strategii dostaliśmy więc wczoraj kolejną składaną w pośpiechu ustawę, wprowadzającą rozwiązania, na które był czas kilka miesięcy temu. Dobrze, że część z naszych poprawek udało się wprowadzić. Wśród nich jest możliwość odmowy sprzedaży w sklepie osobom, które nie chcą zakrywać ust i nosa, czy wykreślenie zapisu o kierowaniu do walki z koronawirusem rodziców małych dzieci. Dobrym rozwiązaniem są wyższe wynagrodzenia dla personelu ochrony zdrowia. Zwykła przyzwoitość każe rekompensować pracę w szczególnie trudnych warunkach, z powodu narażania zdrowia, a nawet życia. Za krok w dobrym kierunku uważamy zapis uzależniający udzielanie pomocy publicznej firmom od tego, czy przestrzegają zaleceń sanitarnych. Od wielu dni bowiem docierają do nas niepokojące informacje o tym, że pracodawcy narażają życie i zdrowie ludzi, ukrywając przed sanepidem przypadki zakażeń. To rozwiązanie nie jest idealne, ale daje jasny sygnał, że takie praktyki nie powinny być dopuszczalne. Niestety odrzuciliście naszą poprawkę gwarantującą 100% wynagrodzenia dla wszystkich pracowników przebywających na kwarantannie. Przyznam, że argumenty przedstawicieli PiS-u, partii podobno prosocjalnej, były zaskakujące. Usłyszeliśmy, że na kwarantannie należy pracować zdalnie, a nie się obijać. Poseł Latos nie uwierzył nam, że nie każdą pracę da się wykonywać w trybie zdalnym. Nie wiem, panie pośle, czy pan kiedyś próbował pracować i jednocześnie opiekować się objętymi tą samą kwarantanną dziećmi. Ja tak. Zapewniam pana, że graniczyło to z cudem. Czyli PiS chce wsadzać lekarzy do więzień i tylko czasowo wprowadzacie abolicję, na czas pandemii. Proszę mi wybaczyć, ale w zapewnienia ministra Gadomskiego, że Zbigniew Ziobro przygotuje wkrótce lepsze przepisy, zdecydowanie nie wierzę. Pan premier apelował o narodową jedność i solidarność. Nie raz szczuliście na lekarzy, na pielęgniarki, na nauczycieli. Mam nadzieję, że dziś zrozumieliście, jak bardzo są potrzebni, jak się poświęcają i jak wielki należy im się szacunek. Część zapisów tej ustawy każe się obawiać, że powoli szykujecie się jednak do przerzucania winy za swoje porażki na pracowników ochrony zdrowia. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Dzisiaj jednak jest jeszcze jedna grupa społeczna, którą chcecie sponiewierać. Dziś wasz niekonstytucyjny trybunał ma wydać wyrok w sprawie możliwości przerywania ciąży w przypadku ciężkich wad płodu.

Tak się składa, że wśród pielęgniarek, lekarzy i nauczycieli większość to kobiety.

Dziękuję, pani poseł. Pan poseł Jan Szopiński, klub Lewica. Wysoka Izbo! Tworzenie przepisów przeciwepidemicznych dopiero w czasie pandemii jest kolejnym przykładem tego, że rząd szuka miejsca na studnię dopiero wtedy, gdy wszystko się pali i wali. W dodatku nie zawsze szuka tam, gdzie powinien. Miejscem, gdzie nie powinien szukać, jest ustawa, która mówi o zwiększeniu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o dwoje dyrektorów. My się tego nie domagaliśmy. My domagamy się tego, aby były w Państwowej Inspekcji Sanitarnej dodatkowe zatrudnienia, aby było dodatkowe wynagradzanie pracowników, aby były skierowane tam osoby, które są zwalniane z administracji państwowej. Czy rząd od wiosny nie nauczył się niczego na swoich błędach?

I w tym zakresie składamy na ręce pani marszałek poprawki. Składamy również poprawkę (Dzwonek), która mówi o 150% przeciętnego wynagrodzenia we wszystkich jednostkach służby zdrowia na czas trwania pandemii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 głos zabierze pan poseł Dariusz Klimczak. Wysoka Izbo! Ta ustawa nie jest cudownym lekiem na wszystkie problemy, które wynikają z epidemii trwającej w naszym kraju, ale jest ratowaniem sytuacji i nadrabianiem strat w zakresie uzupełniania decyzji, które powinny zostać podjęte jakiś czas temu. Dotyczyło to każdego klubu, także posłów, posłanek niezrzeszonych.

To, że została przyjęta ta poprawka, także z rekomendacji, z poparciem rządu, było zaskakujące, ale dobre. Natomiast już dzisiaj po analizie tego przepisu widzimy, że jeżeli dalej będzie dobra wola wszystkich klubów i rządu w tej kwestii, to warto to jeszcze poprawić w Senacie. Mianowicie chodzi o tę część, która dotyczy strażaków ochotników, którzy wykonują zawód rolnika. Tutaj na pewno należy dokonać pewnych zmian, żeby wszystkie te zawody były równe, równo traktowane. Będziemy nad tym pracować i liczymy na taką samą przychylność jak przy pracy w komisji, także - mam nadzieję - w głosowaniu. Oczywiście zależało nam jako klubowi Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 na tym, aby wszystkie zawody, które walczą z epidemią, były w ten sam sposób traktowane, w ten sam sposób premiowane. Stąd zgłoszenie naszej ustawy dotyczącej premii dla bohatera. Jest ona we wnioskach mniejszości i prosimy o poparcie. Uważamy, że trzeba zwrócić uwagę na wszystkich, także na szary personel, który chodzi po tych szpitalach, chodzi po tych podmiotach leczniczych i tak samo jest narażony na zakażenie. To są osoby, które wykonują prace elektryczne, to są wszyscy ci, którzy dbają o to, aby ten podmiot leczniczy funkcjonował. O nich pamiętamy, o tych ludziach pamięta klub Koalicji Polskiej - Polskiego Stronnictwa Ludowego - Kukiz15. Bardzo prosimy o to, aby nasze wnioski poprzeć. W naszych poprawkach upominaliśmy się o kwestie, na których zależało m.in. ogólnopolskiemu związkowi pielęgniarek i położnych, samorządowi lekarskiemu.

O to lekarze zabiegają. Kwestia uregulowana w tej ustawie, nazwana klauzulą dobrego samarytanina, nie załatwia tego problemu, który jest sygnalizowany od samego początku. Chcielibyśmy także, aby prywatny system ochrony zdrowia został włączony do walki z epidemią. Mało tego, chcielibyśmy, żeby ludzie, którzy nie mogą w normalny sposób dostać się do lekarza i się leczyć, mieli także możliwość skorzystania z tego.

Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Krzysztof Paszyk, również klub parlamentarny Koalicja Polska. Bardzo dziękuję. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Myślę, że ta wczorajsza debata i atmosfera ostatnich godzin i dni pokazały, że jeszcze wiele przed nami, jeśli chodzi o pewną weryfikację postaw. Dzisiaj wszystkie stronnictwa reprezentowane w Sejmie powinny identyfikować jednego wroga. Wróg jest jeden, ten wróg to dzisiaj grożący Polsce koronawirus.

Myślę, że to jest dzisiejsza lekcja, która płynie z prac nad tą ustawą, ale też z pewnych niedociągnięć, które były z nami w ciągu ostatnich tygodni czy miesięcy, ale nie ma sensu do tego wracać. Dzisiaj przed nami kolejne tygodnie, miesiące walki z pandemią. Dziękuję bardzo. W imieniu Koła Poselskiego Konfederacja zdalnie głos zabierze pan poseł Janusz Korwin-Mikke. Czy mamy połączenie? Jest. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

W szkołach zawodowych i specjalnych uzależnia się to od decyzji dyrektora. Wykonanie powierza się ministrowi edukacji i nauki. Istota tej ustawy jest oczywista. Podział na płcie zmniejszy interakcję między uczniami, co znacznie zmniejszy możliwość zarażenia się koronawirusem i przenoszenia koronawirusa między uczniami. Ale ma to również aspekt dalekosiężny.

Dziękuję, panie pośle.

To jedna z kilkunastu poprawek, które składamy w tym drugim czytaniu - mamy nadzieję, że nie zostaną one, tak jak poprzednie 16 poprawek, odrzucone przez Wysoką Izbę - również w zakresie walki z koronawirusem czy walki ze skutkami polityki rządu. Proszę państwa, na świecie tak naprawdę są dwa modele, które zostały zastosowane przez państwa wobec epidemii koronawirusa. Pierwszy model to model chiński.

Chińczycy na początku tej epidemii zamknęli kilkadziesiąt milionów ludzi i teraz stosują bardzo daleko posunięte restrykcje, tylko że Chiny liczą sobie 1400 mln ludzi i mogą sobie pozwolić na takie działania. Właściwie żadne inne państwo na świecie na takie działania pozwolić sobie nie może, niezależnie od tego, czy jest to polityka sensowna, czy koszty tego nie przewyższają zysków.

Otóż od początku Konfederacja mówi jasno, że trzeba skoncentrować się na trzech rzeczach. Po pierwsze, na ochronie najsłabszych i najbardziej zagrożonych, czyli seniorów i tych, którzy są chorzy, których odporność jest z jakichś powodów strukturalnie bardzo obniżona. Po drugie, na pełnym wsparciu systemu ochrony zdrowia.

A państwo działają zupełnie na odwrót. Państwo działają w ten sposób, że system ochrony zdrowia przez pół roku nie został przygotowany na tę jesień. Myśmy o tym mówili, że będzie katastrofa. Wokół każdego przypadku pozytywnego testu na koronawirusa jest taka sytuacja, jaką państwo dzisiaj stworzyli. Chodzi o i tak niewydolny system ochrony zdrowia, za co odpowiedzialność ponosi nie tylko PiS, ale i SLD, które dzisiaj chce kneblować debatę na ten temat, i Platformę, która rządziła tyle lat.

W czym gorsi od chorych na COVID są ludzie, którzy dzisiaj umierają, bo nie dostają opieki ze względu na choroby serca, ze względu na nowotwory, na szereg innych chorób, które codziennie zabijają tysiące ludzi, i to nie w skali miesiąca czy dwóch, tylko codziennie? Jeśli pan premier chce debatować, to proszę rozpocząć tę prawdziwą debatę. Prawdziwa debata na temat koronawirusa to debata również o tym, co się dzieje w Szwecji, jaką drogą idzie. To jest debata na temat kosztów, również kosztów życia ludzkiego, nie tylko gospodarczych, ale kosztów życia ludzkiego, bo musimy chronić najsłabszych, całą energię koncentrować na systemie ochrony zdrowia i zarabiać pieniądze.

Przechodzimy do pytań. Wyznaczam czas na zadanie pytania - 1 minuta. Jako pierwszy pytanie zada pan poseł Marek Sowa, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wśród kluczowych poprawek odrzuconych przez polityków Prawa i Sprawiedliwości jest poprawka zapewniająca gwarancję ustawową 200-procentowego wynagrodzenia dla wszystkich pracowników medycznych - lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych - zatrudnionych na pierwszej linii frontu w walce z COVID-19.

Dzisiaj jest on wypłacany na podstawie polecenia ministra. Ale, szanowni państwo, los pracowników służby zdrowia nie może zależeć od jednego podpisu ministra. Musimy mieć gwarancje ustawowe.

Bardzo proszę.

Wysoka Izbo! Ogromne wrażenie wywarło na mnie spotkanie z zarządem świętokrzyskim Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Środowisko pielęgniarskie jest głęboko zaniepokojone planem transferu środków z OWU, tzw. zembalowych, do ogólnej puli środków przekazywanych pracodawcom za świadczenia medyczne. Armii pielęgniarek i położnych pracujących ponad siły Ministerstwo Zdrowia może w konsekwencji zmniejszyć wynagrodzenia w szczycie zachorowań nawet o 1/3. Moim zdaniem powinny zarabiać co najmniej średnią krajową. Pytam zatem: Czy chcecie oszukać te dzielne kobiety? Pan premier Morawiecki mówił o wyimaginowanych liniach obrony zdrowia Polek i Polaków. Przecież rząd PiS zrujnował w ciągu ostatnich miesięcy wszystkie linie obrony. Reszta może się nie doczekać. Zafundowaliście nam wariant szwedzki bez przygotowania i bez znieczulenia. Wysoka Izbo! Wracam do tematu zaangażowania prywatnego systemu ochrony zdrowia w leczenie w trakcie epidemii koronawirusa.

Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kłaniam się.

Chłopcy i dziewczynki w innym tempie rozwijają swoje zdolności.

Bardzo proszę. Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Tych wszystkich problemów nie rozwiążemy pewnie tym projektem ustawy, co jest oczywiste, natomiast możemy zapewnić bezpieczeństwo przynajmniej konkretnej grupie osób.

Czy przychylą się państwo do 100-procentowego zasiłku wypłacanego z FUZ pracownikom ochrony zdrowia od pierwszego dnia izolacji albo kwarantanny, niezależnie od formy współpracy, np. [[Dzwonek]] także tym, którzy pracują na kontraktach?

Taki plan miał powstać.

Wysoka Izbo! Od dłuższego czasu jestem zasypywany pytaniami od pracowników domów dziecka, od wychowawców z ośrodków szkolno-wychowawczych.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.

Tworzycie procedury, które wyolbrzymiają tę pandemię w tabelkach.

Przecież gdybyśmy analogicznie postępowali w odniesieniu do grypy, anginy, przeziębienia, to mielibyśmy takie same statystyki dotyczące zgonów i zachorowań na anginę, grypę itd. Nadmuchujecie go do takich rozmiarów, że zatraciliście już prawdziwe proporcje i skupiliście całą uwagę na jednym zagrożeniu, lekceważąc wszystkie pozostałe. Czemu tak robicie? Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Mirosław Suchoń, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję. Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

To spowoduje kolejne dni chaosu. Dlatego złożyliśmy poprawki wzmacniające powiatowe i wojewódzkie inspekcje sanitarne zarówno finansowo, jak Rząd mówi, że to im się nie podoba. Panie ministrze, to jaka jest tu alternatywa? Bo powiedzieć: nam się nie podoba, jest bardzo prosto, ale te instytucje potrzebują wzmocnienia już dziś, a tego brakuje. Za to znajdują się przepisy, pod którymi podpisuje się także skrajna Lewica, np. o podwójnym karaniu przedsiębiorców, co w czasie epidemii będzie podwójnie zabójcze. Jak chcecie ratować gospodarkę, skoro takimi przepisami, podwójnym karaniem dobijacie ludzi przedsiębiorczych i aktywnych? To się po prostu nie uda.

Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam dwa pytania.

Panie ministrze, wiele tysięcy ludzi pracuje w służbie zdrowia od początku epidemii, od marca. Nie ma w tych rozwiązaniach konkretnego wsparcia dla tych grup, które każdego dnia narażają swoje życie i zdrowie. My zaproponowaliśmy premię dla bohatera. Szanowni Państwo!

Szanowna Pani Marszałek!

Pan premier powiedział, że zastanawia się i będzie rekomendował to, żeby cała Polska stała się czerwoną strefą. Jest takie powiedzenie, że jak się kłamstwo powtórzy tysiąc razy, to ono staje się prawdą, więc rozumiem, że pan premier zdążył już kilka tysięcy razy powtórzyć zdanie: to nie jest lockdown. Zamykacie państwo sauny, solaria, baseny, siłownie, ponieważ tam gromadzą się ludzie.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Panie Ministrze! Dwa największe grzechy tej ustawy, grzechy naprawdę bardzo ciężkie i bardzo poważne. Po pierwsze, kompletnie zaniedbaliście personel medyczny, który pracuje na kontraktach. Dzisiaj ratownik medyczny, który stara się ratować nasze życie i trafi na kwarantannę, a pracuje na kontrakcie, nie ma złotówki za czas izolacji czy też później choroby. I zdarza się, że najpierw ma 10 dni kwarantanny, potem 10 dni spędza po prostu na chorobowym, a pracując na kontrakcie, ubezpieczenie chorobowe dostaje dopiero po 30 dniach. I naprawdę, panie ministrze, trzeba to zmienić, jeżeli chcemy mieć ludzi, którzy będą ratować nam życie w tym trudnym czasie. Nie macie pomysłu, jak to zrobić, a stało się tak, że sanepid stał się wąskim gardłem, nie mają tam nawet czasu na uzupełnianie bazy danych. Musicie też dofinansować sanepid i musicie zadbać o to, by uzupełnić w nim wakaty. W Wielkopolsce jest pilnie dziś potrzebnych 30 dodatkowych par rąk do pracy, których nie ma. Pan poseł Jacek Protas, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pan premier wczoraj w płomiennym wystąpieniu zachęcał wszystkich do współpracy w tym trudnym, pandemicznym okresie - trudnym dla nas wszystkich. To słowa. A czyny? Otóż proponuje w ustawie zapisanie dla ministra zdrowia prawa do odwoływania, arbitralnie, dyrektorów szpitali - dyrektorów szpitali, które podlegają samorządowi terytorialnemu. Czy to jest wyciągnięcie ręki do współpracy?

Wysoka Izbo! Rzeczywiście ten projekt ustawy ma poprawić funkcjonowanie ochrony zdrowia, ale jest pytanie, czemu państwo nie chcecie wprowadzić tych dodatków i wynagrodzeń dla ludzi, którzy są na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem i są najbardziej narażeni na potencjalne zagrożenie, czyli pracowników SOR-u, pracowników izby przyjęć, pracowników pogotowia, laborantów. W związku z tym moje pytanie jest takie: Czy przewidujecie w tej sytuacji zmianę w budżecie państwa na rok 2020? Bo jeszcze raz chcę podkreślić: dzisiaj mamy wojnę z koronawirusem, nie z żadnym najeźdźcą zewnętrznym, tylko wojnę z koronawirusem, i być może warto środki przekazać przede wszystkim właśnie na walkę z pandemią, a nie na kupowanie czołgów, samolotów, armat i pistoletów, bo to dzisiaj nam do niczego nie jest potrzebne.

Dziękuję. Kolejne pytanie zada pani poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę, pani poseł. Dziękuję bardzo. Panie i Panowie Posłowie! Panowie Ministrowie! Wczoraj pan premier wyciągał rękę do opozycji, dziś w nocy większość parlamentarna odrzuciła większość poprawek opozycji. Wczoraj pan premier zapowiadał stworzenie jakiegoś enigmatycznego korpusu ochrony seniorów, dzisiaj seniorzy, tak jak od paru miesięcy, umierają ze strachu w swoich domach, bo powiedziano im, by tych domów nie opuszczali. Umierają ze strachu, czy przyjedzie do nich karetka, czy przyjedzie do nich lekarz, czy znajdzie się dla nich miejsce w szpitalu, gdy dostaną udaru, zawału albo po prostu, jak to bywa u starszych ludzi, nastąpi nagły skok ciśnienia. Wczoraj mówiono tutaj bardzo dużo, że opozycja to politykierstwo, a większość sejmowa to merytoryczna praca. No i w ramach tej merytorycznej pracy dzisiaj pan poseł Piecha składa wniosek, żeby niezwłocznie przejść do trzeciego czytania, bez znajomości poprawek, jakie padły i w nocy, i w drugim czytaniu. Dziękuję, pani poseł. A jeszcze bym bardzo prosiła naszych drogich parlamentarzystów, aby te rozmowy przenieść w kuluary, bo to bardzo przeszkadza, utrudnia pracę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie pośle. Wysoka Izbo! Można by zadać pytanie: Skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? Pacjenci, szczególnie oddziałów onkologicznych, którzy dzisiaj są najbardziej narażeni na COVID, niestety nie mają w miejscu swojego zamieszkania dostępu do niektórych usług. Obiecany kontrakt, który miał być podpisany ze szpitalem w Zgorzelcu na radioterapię, niestety nie doszedł do skutku. Może takimi rzeczami właśnie też powinniśmy się zajmować, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim tym, którzy chorują nie tylko na COVID, ale też na inne choroby. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Może zamiast samolotów dla wojska zmodernizujemy to Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, kupimy śmigłowce, którymi będziemy mogli transportować chorych, tak że osoby z Jeleniej Góry będą mogły się dostać w miarę szybko do Wrocławia, bo dzisiaj, tylko dlatego że państwo nie budują jakichkolwiek dróg i nie szukają rozwiązań, żeby dotrzeć karetką z Jeleniej Góry, o ile autostrada nie stoi, trzeba 2 godzin. Dlatego apeluję: zróbmy coś dla tych ludzi, którzy chorują nie tylko na COVID. Dziękuję bardzo. Pani poseł Klaudia Jachira, Koalicja Obywatelska. Panie Przewodniczący komitetu do spraw bezpieczeństwa narodowego i spraw obronnych! Wysoka Izbo! Przez pół roku zrobiliście dużo niepotrzebnych rzeczy. Walczyliście z plagą LGBT, ścigaliście niezależnych sędziów, adwokatów, zajmowaliście się wyborami, walką o stołki, zakazem aborcji i finansowaniem propagandy sukcesu, podczas gdy wirus rozlewał się po kraju. Dlaczego nie zrobiliście jednej rzeczy, którą zrobiły takie kraje, jak Korea Południowa i Norwegia, którym udało się opanować epidemię? Nie zrobiliście powszechnego, darmowego testowania, które wykrywa bezobjawowe ogniska wirusa. Musi dzwonić do jednego, drugiego lekarza, może mu ktoś łaskawie pozwoli, a na koniec i tak pójdzie prywatnie, zapłaci, a wy tego wyniku nie ujmiecie w statystykach. Swoją opieszałością i zaniedbaniem doprowadziliście do tego, że teraz będą umierać tysiące Polek i Polaków. Zamiast słuchać Trumpa, warto czasem posłuchać WHO. Pan poseł Paweł Krutul, klub Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dlatego jako reprezentant województwa podlaskiego zwracam się do pana premiera, pana ministra, wojewody województwa podlaskiego pana Paszkowskiego o otwarcie trzech szpitali polowych w największych miastach województwa, tj. w Białymstoku, Suwałkach i Łomży. Do zagospodarowania są hale sportowe, stadion miejski czy też ewentualnie ośrodki wczasowe, które teraz w województwie podlaskim świecą pustkami. Tak że proszę o jak najszybsze utworzenie tych miejsc, żeby przede wszystkim wdrożyć profilaktykę i odciążyć jednostki, które teraz zajmują się osobami chorymi na COVID. Dziękuję bardzo. Pan poseł Cezary Grabarczyk, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Skuteczna walka z pandemią będzie zależała od skutecznej strategii. Rząd postawił na strategię gigantomanii, pewnych pokazowych akcji. Wiosną to był gigantyczny Antonov z maseczkami, które okazały się nieprzydatne, a dziś czytamy artykuł i być może rząd będzie musiał się za to wstydzić. Teraz jest mowa o szpitalu na Stadionie Narodowym i to jest kolejny przykład gigantomanii. Tymczasem trzeba postawić na siły społeczne. Są oferty: tu możecie stworzyć miejsca dla chorych - mówi o tym prezydent Warszawy. Nie chcecie wysłuchać opozycji, która prawie jednym głosem mówi: postawcie na kapitał ludzki, dajcie podwójne wynagrodzenia lekarzom, [[Dzwonek]] postawcie na ubezpieczenia. Upominamy się o to. Pani poseł Marta Wcisło, Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! Dosyć tych kłamstw, że przygotowaliście kraj na walkę z epidemią. To nieprawda. Sytuacja jest dramatyczna. Już dziś pacjenci umierają w karetkach, które jeżdżą od szpitala do szpitala, odbijają się. Brakuje respiratorów. Już dziś pacjenci czasowo są odłączani od urządzeń po to, żeby podłączyć innych. U handlarza bronią? Podejmujecie decyzje nielogiczne. Otworzyliście szpitale jednoimienne, które zamknęliście. Teraz otwieracie szpitale polowe. Zaprzepaściliście czas, przehulaliście pieniądze i naraziliście zdrowie pacjentów. Dlaczego do tej pory nie stworzyliście systemu informatycznego, który koordynuje pracę szpitali i relokację zasobów? Dlaczego? Dlaczego za złe decyzje, przehulane pieniądze nie ścigacie swoich kolegów? Wypłaszcza się wasze myślenie i przekształciło się w wirusa, wirusa nienawiści, niekompetencji i niewspółpracy, bo mieliście współpracować, a dzisiaj odrzucacie najlepsze nasze poprawki. 90% naszych poprawek z pracy nocnej zostało odrzuconych, dobrych poprawek dla obywateli.

Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Uczucia, z którymi budzą się codziennie Polki i Polacy to strach i niepokój o naszych najbliższych. Nasza kontrola z panem posłem Jońskim nie była aktem oskarżenia, była swoistym wołaniem na puszczy. Z posłem Jońskim zadawaliśmy pytania nieustannie, gdzie są respiratory, dlaczego przepłacacie, dlaczego za cenę dwóch respiratorów kupujecie jeden, dlaczego nie testujecie DPS-ów, gdzie jest strategia. Dzisiaj dowiadujemy się, że powstał okólnik w Ministerstwie Zdrowia, który wysyłał były wiceminister. Tego już więcej nie będzie. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska złożyła poprawkę. Wszystkie zamówienia, które będziecie realizować, będą musiały być zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Będziemy wam patrzeć na ręce i każdą złotówkę zdefraudowaną odkryjemy. Pan poseł Jan Szopiński, klub Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ta ustawa nie rozwiązuje wszystkich problemów polskiej służby zdrowia. Przed rządzącymi pilna odpowiedź na pytanie, co zrobić z pogarszaniem się dostępu pacjentów do świadczeń medycznych. Dostępność specjalistów jest jeszcze gorsza.

Dziękuję bardzo. Pan poseł Piotr Borys, Koalicja Obywatelska.

Szanowna Pani Marszałek! Wczoraj pan premier powiedział nam o tym, że powinniśmy być solidarni w walce z COVID-em. Tymczasem komisja odrzuciła poprawki, które mają wzmacniać sanepid, po to żeby chronił nas przed COVID-em. Odrzuciła przywrócenie handlu w niedzielę, który może uratować tysiące miejsc pracy. Na końcu odrzuciła również poprawki związane z gwarancją 200% wynagrodzenia dla wszystkich pracowników służby zdrowia. Ale odrzuciła również poprawkę, która daje możliwość stworzenia 10-miliardowego funduszu, który pozwoliłby na to, aby powszechnie zaszczepić Polaków przeciwko grypie. Dzisiaj to jest tylko 4% naszych rodaków, a 75% populacji zaleca Unia Europejska. Włochy, Francja szczepią przeciwko grypie 70% swoich obywateli. Dlaczego Polska tego nie zrobiła? Chcę państwu powiedzieć w ostatnim zdaniu, że Polska jest na 24. miejscu w Europie z najmniejszą liczbą testów na milion mieszkańców. Trzeba to zmienić, przyjmijcie nasze poprawki, jeżeli mamy solidarnie walczyć z COVID-em. Pan poseł Tadeusz Tomaszewski, klub Lewica. Wysoki Sejmie! W art. 20 w zmianie piątej przyjęto rozwiązanie, które przewiduje możliwość otrzymania 100-procentowego zasiłku chorobowego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy biorą udział w akcjach ratowniczych i w związku z powyższym mają chorobę COVID lub są na kwarantannie. Natomiast nie przyjęto rozwiązania, które dawałoby taką samą rekompensatę dla członków OSP, którzy są rolnikami i są ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Może tą drogą w trakcie dalszych prac można byłoby to naprawić. Jakie środki finansowe rząd skieruje do szpitali powiatowych w związku z dodatkowymi zadaniami wynikającymi ze zwalczania COVID-19? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Michał Gramatyka, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Czy rząd prowadzi analizy i badania oceny wpływu pandemii na inne niż COVID zagrożenia zdrowotne? Czy ktoś np. bada, jak pandemia rzutuje na zdrowie psychiczne Polek i Polaków? W Polsce rocznie odnotowuje się 6 tys. samobójstw. Kanadyjskie badania nad COVID-owym lockdownem pokazują, że wzrost bezrobocia o 1 punkt procentowy implikuje taki sam wzrost liczby samobójstw. Czy w Polsce są takie badania? Bo państwo, rząd, wzrost bezrobocia planujecie na 5% rocznie. Zamykacie ludziom siłownie i kluby fitness, nie wiadomo po co. Nie było ognisk wirusa w siłowniach, a według amerykańskiej rządowej agencji CDC utrzymanie fizycznej aktywności w czasie pandemii jest pożądane i korzystne dla zdrowia, również psychicznego. Czy ktoś z was myśli o tym właśnie w ten sposób? Pani poseł Paulina Matysiak, klub Lewica.

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Zgodnie z zapisami ustawy izby zawodowe zawodów medycznych mają obowiązek przekazać dane tych swoich członków, którzy mogą być skierowani do walki z koronawirusem. Żeby to ustalić, trzeba zebrać szereg danych, którymi te izby w tym momencie nie dysponują. One już o tym mówiły, zgłaszały to. Zgodnie z ustawą będą miały na to 7 dni. Już teraz wiadomo, że jest to niewykonalne w tak krótkim czasie. Naprawdę uważacie, że te osoby, które mają teraz nas leczyć, mają zająć się zbieraniem danych, wysyłaniem maili i telefonowaniem do swoich członków? Tutaj uwaga: Lewica proponowała już swoje rozwiązania, zaangażowanie w działania walki z pandemią call centers, które mogą wesprzeć sanepidy, ale mogą też być przydatne w takich sytuacjach, jak właśnie ta proponowana w ustawie. Być może wcale nie chodzi o to, żeby kogokolwiek kierować na ten front walki z pandemią, tylko chodzi o to, by przenieść ciężar odpowiedzialności (Dzwonek) na lekarzy, pielęgniarki i inne zawody medyczne.

Wysoka Izbo! Mam bardzo poważną sprawę. Doprowadzicie państwo do tego, że niepełnosprawni będą umierać w swoich domach ze swoimi opiekunami. Dostaję dramatyczne telefony od rodziców, którzy nie mogą zrobić zwykłych zakupów i pójść do lekarza, bo nie mają co zrobić z ciężko upośledzonymi dziećmi, z którymi są w domach. Już od marca MOPS-y w całej Polsce powinny być w kontakcie chociażby telefonicznym z tymi rodzicami, a nie są. Propaganda pana Morawieckiego zgadza się, zgadza się na 100%, ale nie zgadza się z rzeczywistością. A więc bardzo proszę i pytam: Gdzie jest konkretne wsparcie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, dla rodzin, w których są osoby niepełnosprawne? Gdzie jest wsparcie dla rodziców pracujących? Bo są też tacy rodzice [[Dzwonek]] dzieci niepełnosprawnych, którzy pracują. Oni w ogóle. Powinny się znaleźć pieniądze właśnie dla takich rodziców, którzy w heroiczny sposób godzą opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym i pracę. Dziękuję. Pan poseł Tomasz Olichwer, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! W uzasadnieniu ustawy PiS-u napisano, że w czasie epidemii powinno następować wyłączanie odpowiedzialności karnej za określone czyny popełnione przez osoby wykonujące zawód medyczny, gdy działania lecznicze są podejmowane w celu zwalczania epidemii, np. w sytuacji realizacji świadczeń przez osoby, które w warunkach nieepidemicznych nie udzielałyby tych świadczeń. Moim zdaniem te zapisy są mało precyzyjne i mogą spowodować, że będą nas leczyć obok dobrze wykwalifikowanych lekarzy także amatorzy. A przecież jakiś czas temu chcieliście państwo sprowadzać lekarzy z zagranicy. Szanowni Państwo!

Pan poseł Adam Szłapka, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Panie Ministrze! Ten szczególny czas wymaga szczególnych rozwiązań, co rozumiemy, i dlatego nikt z nas nie uchylał się od ciężkiej pracy w komisji przy tej ustawie. Natomiast rzeczą absolutnie niedopuszczalną jest wykorzystywanie tej szczególnej sytuacji do wprowadzania rozwiązań, których celem jest rozwiązywanie kwestii personalnych. Nie da się niczym uzasadnić wpisywania do ustawy możliwości podejmowania arbitralnej decyzji przez ministra, jeśli chodzi o odwoływanie dyrektorów szpitali wszystkich szczebli, także szpitali samorządowych. Wszyscy są zaangażowani w walkę z pandemią: medycy, lekarze, samorządowcy, dyrektorzy szpitali. A wy chcecie wprowadzić rozwiązanie, które pozwala arbitralnie usunąć dyrektora szpitala. To jest rozwiązanie niedopuszczalne, tak jak niedopuszczalne było wykorzystywanie tej sytuacji przy tego typu zakupach [[Dzwonek]] maseczek czy respiratorów. Dziękuję bardzo. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Na postawione pytania odpowie w pierwszej kolejności podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia pan Sławomir Gadomski. Panie ministrze, bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Po pierwsze, chciałem złożyć serdeczne podziękowania za wczorajszą pracę, podziękowania być może najpierw na ręce wnioskodawców tego projektu kluczowego, nad którym pracowaliśmy, ale i na ręce wszystkich wnioskodawców, bo wydaje mi się, że istotną część z tych projektów złożonych przez opozycję, istotną część rozwiązań również wdrożyliśmy, w przypadku projektu Lewicy wdrożyliśmy praktycznie całą ustawę w treść ustawy zaproponowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Tego dzisiaj być może z tej mównicy nie widać, rozumiem, że na tej mównicy trochę inny charakter wypowiedzi muszą albo chcą państwo stosować, jednak wczorajsza współpraca była konstruktywna, rzeczywiście tak ją odbieram. Mieliśmy dosyć dużo czasu na merytoryczną dyskusję i za tę dyskusję serdecznie dziękuję. Największą energię na tej mównicy teraz, podczas zadawania pytań, wykazali posłowie, których wczoraj nie było niestety z nami. No, rozumiem, wyspali się, mieli dosyć dużo czasu na przygotowanie się do tych pytań i wykazania tej energii. Martwi mnie, że właśnie tych, których nie było, dalej nie ma. Szanowni Państwo! Krótkie odniesienie się jeszcze do wypowiedzi i dyskusji, bo myślę, że to również da podkład, da fundament do odpowiedzi na pytania szczegółowe. Wynagrodzenia lekarzy.

Ta ustawa zwiększa wynagrodzenia o 100%, czyli do 200%, lekarzom, którzy są delegowani przez wojewodów do pracy.

Teraz również te polecenia, które wydawał minister zdrowia, które były realizowane przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zostaną zmienione i te 200% ci lekarze, którzy włączyli się do walki, czy personel medyczny, który się włącza, oczywiście otrzymają. Szanowni państwo, nie potrzebujemy dodatkowego funduszu. Część, istotną część tego funduszu do dyspozycji otrzymał minister zdrowia, praktycznie tę część, można powiedzieć, nieograniczoną. Oczywiście mamy zaplanowane, że na ten rok to jest 10 mld, ale non stop konsultując i uzgadniając dalsze transze z tego projektu, jednoznacznie mamy zapewnienie, że będziemy mogli korzystać według naszych potrzeb. Tak że tutaj nie ma potrzeby tworzenia dodatkowego funduszu, bo my więcej w tym funduszu, który mamy, mamy już dzisiaj w tych planach, na następny rok również. Szanowni państwo, to rozwiązanie, które wprowadziliśmy w ustawie, to rozwiązanie, o którym tak dużo wczoraj dyskutowaliśmy, jest zgodne i spójne z intencją, z tym, czego oczekiwała Naczelna Rada Lekarska w zakresie wyłączenia skutków Kodeksu karnego na czas pandemii. Tak że wydaje mi się, a nawet jestem przekonany, że rzeczywiście realizujemy postulaty środowiska w tym zakresie.

System prywatny już dzisiaj zadeklarował włączenie się, zadeklarował włączenie się do walki z COVID, zadeklarował, że jest w stanie np. w zakresie szpitali prywatnych przeznaczyć nawet 1/4 łóżek na walkę z COVID-em. Rozumiem, że ta dyskusja dotyczy czego innego, czyli wsparcia przez system prywatny leczenia nie-COVID-owego. Wydaje mi się, że rozwiązanie zaproponowane przez państwa jest bardzo szerokie, jest trudne do wdrożenia.

Myślę, że to rozwiązania, nad którymi można (Dzwonek) dyskutować, ale chyba nie w tym trybie, w którym dzisiaj jesteśmy, i nie w trybie tej ustawy, która jak wszyscy chyba się zgadzamy, jest odpowiedzią na sytuację, którą mamy. Szanowna pani marszałek, czy mogę skorzystać. Padło wiele pytań, każdy jest zainteresowany odpowiedziami.

Wiemy dobrze, że część służby zdrowia pracuje w takiej formule, ale też wiemy dobrze, że był to wybór tych osób.

Ochrona tych osób w stosunku do osób zatrudnionych na umowę o pracę jest w naturalny sposób mniejsza.

Pan poseł Sośnierz pytał o statystyki dotyczące zgonów. Od początku nie chcemy przekłamywać i nie chcemy udawać dzisiaj, że COVID nie ma i zgonów na niego nie ma. Podjęliśmy próbę określenia pewnych wymagań, wymagań, których nie określiliśmy sami w urzędzie, tylko oczywiście wypracowaliśmy je wspólnie z ekspertami, z konsultantami krajowymi. Ich stanowisko było takie, że jeżeli mamy np. chorobę wieńcową i COVID dodatni to jednak wykazujemy to jako COVID dodatni. Czy chcemy z tym dzisiaj dyskutować? Ważne, że te statystyki są pokazywane rzetelnie, spójnie i zgodnie rzeczywiście z tymi opublikowanymi zasadami. Nie chcemy podwójnie karać przedsiębiorców, w ogóle nie chcemy ich karać. Jeżeli tylko ci przedsiębiorcy będą przestrzegać nakazów, zakazów, które wprowadzamy na poziomie uchwał Rady Ministrów czy rozporządzeń ministra zdrowia, to żadnych kar nie będzie. To jest jedynie, można powiedzieć, pewna sankcja, którą rzeczywiście widzimy jako logiczną kontynuację. Jeżeli państwo wspomaga wiele przedsiębiorstw tarczą antykryzysową, jeżeli te przedsiębiorstwa mogą otrzymywać dodatkową pomoc publiczną, to nie możemy przymykać oczu na nieprzestrzeganie tych zakazów, których przestrzeganie jest dzisiaj ekstremalnie ważne dla całego systemu ochrony zdrowia. Pani poseł Hennig-Kloska pytała m.in. o niedofinansowanie sanepidu. Tego systemu zmieniać nie trzeba.

Na przyszły rok, czyli od stycznia następnego roku. Chcę też zauważyć, że w tym roku również duże środki na finansowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w szczególności np. na wypłatę wynagrodzeń dodatkowych za nadgodziny, są realizowane, na wyposażenie czy na infrastrukturę w sanepidach, od samego początku te środki są tam kierowane. Kilka pytań, jak dobrze pamiętam, pana posła Protasa i pana posła Szłapki dotyczyło odwoływania dyrektora. Nie mówimy o odwoływaniu. Po pierwsze, mówimy o zawieszaniu, i to tylko na czas pandemii.

Ta sankcja, ten przepis funkcjonował od początku pandemii. Ten przepis był już w poprzednich ustawach anty- COVID-owych i do tej pory minister zdrowia nie wykazał aż takiej determinacji, żeby z tego korzystać. Również dlatego, bo pytanie dotyczyło tego, ilu dyrektorów za chwilę wymienimy, nie wymieniliśmy w pół roku żadnego, bo nie widzieliśmy przesłanek, żeby z tego przepisu skorzystać. Mamy nadzieję, że nie zobaczymy tych przesłanek i rzeczywiście świadczeniodawcy będą realizować te wymogi prawa i te polecenia, które zostały wprowadzone. Nawołuję też do pewnej spójności w ramach pytań, bo wydaje mi się, że to jest tak trudny obszar, że same głosy są ekstremalnie różne. Pan poseł Grabarczyk mówił o tym, czy nie jest gigantomanią budowanie szpitala na narodowym, a chwilę wcześniej poseł Krutul wnioskował o wybudowanie trzech szpitali polowych na Podlasiu.

Kilka pytań dotyczyło infrastruktury do testowania i realizacji testów na większą skalę. Chciałbym zwrócić uwagę na jedno: my nie dlatego nie realizujemy być może 100, 200 tys. czy pół miliona testów dziennie, bo brakuje nam na to środków, bo środki na to mamy.

Te założenia nie są wynikiem dyskusji wewnętrznej urzędników w Ministerstwie Zdrowia, tylko dyskusji z konsultantami, dyskusji z konsultantem krajowym prof. Horbanem, dyskusji z konsultantem krajowym panią prof. Dzierżanowską-Fangrat, z wieloma innymi konsultantami, z którymi rzeczywiście od samego początku pandemii pracujemy, i co więcej - jesteśmy przekonani do celności naszej strategii testowania.

Szanowni Państwo! Były jeszcze dwa pytania, jedno zadał pan poseł Tomaszewski - przepraszam, drugiej nie jestem w stanie teraz odnaleźć - o środki dla szpitali powiatowych i finansowanie tych szpitali w tym trudnym czasie.

Szanowna pani marszałek, bardzo dziękuję za przedłużenie. Jeszcze raz dziękuję za wczorajszą pracę i mam nadzieję, że w podobnym duchu będziemy pracowali dalej. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Głos zabierze sprawozdawca komisji pan poseł Tomasz Latos. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Odpowiadając panu posłowi Tomaszewskiemu: tak, rzeczywiście pojawiła się taka poprawka w czasie prac komisji i my po analizie uznaliśmy, że warto ją poprzeć, podobnie jak wcześniejszą poprawkę zgłoszoną z kolei przez Koalicję Obywatelską, która dotyczyła straży miejskiej. Wydawało się, że jest to rozsądne, więc odpowiadając na pytanie pana posła dotyczące OSP: niewątpliwie trzeba teraz pójść dalej, czyli jeszcze dostosować to do innych przepisów, stąd uwaga dotycząca KRUS-u jest w pełni zasadna. Natomiast, szanowni państwo, patrząc na to wszystko, co działo się wczoraj, i wnosząc z tego, co działo się dzisiaj, to powiem szczerze, że jestem w lekkim szoku, mimo że po tylu latach w Sejmie właściwie już nic nie powinno mnie zdziwić.

Ja myślę, że o prawdziwych rzeczach to mówił już pan minister, bo o tych nieprawdziwych może nie warto mówić.

Cóż, taki mamy klimat można powiedzieć, cytując pewną znaną panią minister. Uważam, że coś takiego jak dżentelmeńska umowa jest sprawą niezwykle ważną. Poprawka Lewicy, dwie poprawki, rozumiem, coś zostało jeszcze zauważone, warto skorygować.

Wszystko, co można było zgłosić, zgłaszaliśmy wczoraj.

Myślałem, że w polityce pewne ogólne zasady też powinny obowiązywać, jak się ludzie na coś umawiają, to powinni tego dotrzymywać. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zamykam dyskusję. W trakcie dyskusji złożono wniosek, aby Sejm przystąpił do trzeciego czytania bez odsyłania projektu ustawy do komisji, oczywiście po doręczeniu zestawienia poprawek. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Jest sprzeciw, tak? W takim razie będziemy głosować nad tą sprawą w bloku głosowań, a w tej chwili ogłaszam przerwę do godz. 13.30. Przerwa? Ale sprostowanie do czego, panie pośle? Pan przewodniczący był uprzejmy powiedzieć, że była jakakolwiek umowa. A nie dość tego. Nie było żadnej umowy, absolutnie. Poprawki były, natomiast były uzgodnienia, że nie będziemy przekazywać tego do komisji. Ale przepraszam bardzo, ogłosiłam przerwę. Przenieście państwo uzgodnienia w kuluary.

Wznawiam obrady. Przystąpimy obecnie do stwierdzenia kworum. Proszę o wciśnięcie dowolnego przycisku w celu potwierdzenia obecności na posiedzeniu.

Głosowało 449 posłów. Stwierdzam kworum. Pan poseł Cezary Tomczyk, Koalicja Obywatelska.

To jest sytuacja, z którą mamy do czynienia. To jest kpina z państwa, z Polaków i z tego wszystkiego, co się dzieje. Mniej testów, więcej zachorowań. Wysoka Izbo! Jeżeli chodzi o kwestię tej ustawy, widać ponad wszelką wątpliwość, że warto było nad nią pracować.

Dzięki poprawce Koalicji nie będzie już można kupić respiratorów od handlarza bronią. dlatego że wszystkie transakcje będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pani poseł Barbara Nowacka, Koalicja Obywatelska. Wysoki Sejmie! Prosimy o uzupełnienie porządku obrad o informację pełnomocnika rządu ds. równego traktowania. W tej chwili obraduje tzw. Trybunał Konstytucyjny i ma wydać wyrok na kobiety.

Nie mieliście odwagi dyskutować o tym z mównicy sejmowej, miejcie odwagę wezwać pełnomocniczkę.

Wysoka Izbo!

Pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz od ponad 2 miesięcy oczekuje na procedurę, w której będziemy mogli głosować i dowiedzieć się, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie jako Wysoka Izba wybrać następcę Adama Bodnara. Te kilka. Panie pośle, pan się orientuje, że to jest wbrew regulaminowi?

Prosiłbym, panie marszałku, żebyśmy jednak przegłosowali to, dlatego że wysłuchanie.

Składam wniosek o przerwę. Przerwa może być krótka, pod warunkiem że pan wicepremier Jarosław Kaczyński, przewodniczący komitetu do spraw bezpieczeństwa, przyjedzie tutaj i wytłumaczy nam, jakie działania podejmuje rząd w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego kraju spowodowanego straszliwą ustawą antyrolniczą, piątką antyrolniczą, którą pan Kaczyński forsuje dzisiaj przez Sejm. Wczoraj tysiące rolników protestowało na polskich drogach przeciwko temu bezprawiu, przeciwko temu łajdactwu, które państwo, koalicja PiS, Platforma, SLD, próbujecie przeprowadzić wobec polskiej wsi.

Rozumiem, że są wnioski o przerwę. A więc będziemy głosować niestety wniosek o przerwę, co wydłuży głosowania. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, zechce nacisnąć

Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat stanu przygotowania państwa na rosnącą falę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i wywoływanej nim choroby COVID-19, a także wirusa grypy w czasie pandemii koronawirusa. W dyskusji złożono wniosek o odrzucenie przedstawionej informacji, który poddam pod głosowanie. Odrzucenie tego wniosku będzie oznaczało, że Sejm przyjął informację do wiadomości. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie informacji prezesa Rady Ministrów, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek przyjął. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 698. Komisja przedstawia również wnioski mniejszości, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

W 4. wniosku mniejszości wnioskodawcy proponują skreślić art. 2. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Przyjęcie tego wniosku spowoduje bezprzedmiotowość 7. wniosku mniejszości. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 7. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wniosek odrzucił.

Kto się wstrzymał?

Nad tymi wnioskami będziemy głosować łącznie. Kto jest przeciw?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 11. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił.

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 12. wniosku mniejszości i 1. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Kto jest przeciw?

Sejm propozycje odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 15. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 16. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 19. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 20. wniosku mniejszości i 3. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 21. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wniosek odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 34. wniosku mniejszości? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. W 10. poprawce wnioskodawcy proponują skreślić art. 19. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 10. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił.

Kto jest przeciw?

Sejm wniosek odrzucił.

Sejm wniosek odrzucił.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 37. wniosku mniejszości? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 11. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 39. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Za - 209, przeciw - 229, wstrzymało się 11.

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 12. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Za - 207, przeciw - 231, wstrzymało się 11 posłów. Sejm poprawkę odrzucił. 40. wniosek mniejszości jest bezprzedmiotowy, ponieważ jego treść została już uwzględniona w komisyjnym przedłożeniu projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 41. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk.

Za - 212, przeciw - 229, wstrzymało się 7 posłów.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 13. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił.

Wznawiam obrady. Kontynuujemy rozpatrywanie punktu 6. porządku dziennego. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 42. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 14. poprawki, proszę nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 15. poprawki, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

wniosku mniejszości. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 44. wniosku mniejszości i 16. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 45. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 17. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 18. i 22., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 19. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 46. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw?

marszałek

Sejm wniosek odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 49. wniosku mniejszości i 20. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 21. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 23. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 50. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 53. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk oczywiście. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy.

Wysoka Izbo! To mógłby być bardzo dobry projekt, spóźniony, ale dobry. To mógłby być projekt, który stałby się istotnym elementem, narzędziem dla rządu w walce z pandemią, gdyby został obudowany naszymi poprawkami, które zwiększyłyby fundusz celowy do walki z pandemią, przyznałyby gwarancję 200% wynagrodzenia dla wszystkich pracowników walczących COVID-em, które wspomogłyby organizacyjnie, kadrowo i finansowo sanepidy, które otworzyłyby sklepy w niedzielę, przyznałyby zasiłki opiekuńcze, przywróciłyby możliwość zarządzania szkołami przez dyrektorów i wiele, wiele innych. Niestety wszystkie te poprawki odrzuciliście, co powoduje, że zmiany nie zbudują potrzebnej strategii dla rządu do walki z koronawirusem, strategii przemyślanej, konsekwentnej, oczekiwanej. Dziś, panie pośle, szanowni państwo, zagłosujemy za tym projektem, bo zawiera kilka dobrych zmian, z nadzieją, że ten projekt wróci z Senatu ponownie obudowany naszymi dobrymi poprawkami, a państwo zmienicie zdanie dla dobra obywateli, [[Dzwonek]] dla ich życia, zdrowia i poprawy bezpieczeństwa.

Udało się naprawdę wypracować bardzo wiele niezwykle ważnych i potrzebnych w tej trudnej, COVID-owej rzeczywistości rozwiązań. Naprawdę, szanowni państwo, nie deprecjonujmy naszej wspólnej pracy, naszego wspólnego wysiłku i projektu, który wart jest poparcia, projektu, który przewiduje rozwiązania również na te najgorsze, najtrudniejsze chwile. Oby do nich nie doszło, oby nie trzeba było tych szpitali, które są potencjalnie tworzone, [[Dzwonek]] nie trzeba było nigdy zapełniać pacjentami. Pan poseł z pytaniem? Pan poseł z pytaniem. Wysoka Izbo! Tworzenie przepisów przeciwepidemicznych dopiero w szczycie pandemii jest przykładem, że rząd szuka miejsca na studnie, dopiero wtedy, kiedy się pali i wali, i w dodatku szuka nie zawsze tam, gdzie powinien. Klub Lewicy świadomy jest ułomności tej ustawy, natomiast świadomi też jesteśmy, że ta ustawa w znaczącym stopniu poprawia system polskiej ochrony zdrowia, zapewnia dobre warunki materialne lekarzom. Mając nadzieję, że Platforma Obywatelska, że koalicja w Senacie zechce poprawić tę ustawę i że PiS, tak jak to deklarował w trakcie prac nad ustawą w komisji, zechce poprzeć w Senacie nasze wnioski. Pan poseł Jan Szopiński.

Wysoka Izbo! Długo pracowaliśmy nad tą ustawą, wiele rzeczy udało nam się wspólnie poprawić w poprawkach merytorycznych, zgodnie. Tego oczekują od nas Polacy, mimo wielkich różnic, które są tutaj na sali. Ale każdy, kto nie dostał się dzisiaj czy wczoraj do lekarza, oczekuje od każdego z posłów, że dołoży cegiełkę do tego, żeby ten system działał sprawnie. Dzisiaj pan minister zdrowia mówił o tym, że trzeba włączyć prywatną ochronę zdrowia do pomocy w walce z koronawirusem. A ja mam pytanie do pana ministra zdrowia: Czy nie warto się zastanowić, żeby każdy pacjent, który nie dostał się do lekarza na NFZ, mógł pójść i wyleczyć się u prywatnego. i dostać zwrot, refundację za to leczenie? W ten sposób pomożemy wszystkim pacjentom. To jest ważne pytanie od każdego Polaka.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 698, zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

Wysoka Izbo! Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim państwu za tak jednoznaczne ocenienie naszych rozwiązań. Uważam, że to jest bardzo dobry projekt. Nie ma bytów idealnych, ale ten projekt rzeczywiście odpowiada na potrzeby, które związane są z rozwijającą się dynamicznie pandemią. Szczególnie chciałbym podziękować za bardzo merytoryczną pracę w komisji. Zarówno panu przewodniczącemu, panu ministrowi Gadomskiemu, który jest tutaj, na sali, jak i wszystkim posłom opozycji, którzy wczoraj w bardzo merytoryczny sposób mieli realny wkład w te rozwiązania, które dzisiaj zostały przegłosowane. Bo w trakcie posiedzenia komisji były przyjmowane wspólnie rozwiązania dotyczące chociażby 100% rekompensaty dla straży miejskiej, publikowania informacji o postępowaniach zwolnionych z zasad dotyczących zamówień publicznych i inne rozwiązania. Tak że, szanowni państwo, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że to jest preludium do szybkiego przejścia ustawy przez Senat. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 7. porządku dziennego: Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich (druki nr 536, 537, 618 i 618-A)

Sejm powołuje rzecznika praw obywatelskich za zgodą Senatu. Na stanowisko rzecznika praw obywatelskich dwie grupy posłów zgłosiły kandydaturę pani Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. W imieniu grupy posłów z klubu parlamentarnego Lewica kandydaturę przedstawi pan poseł Krzysztof Śmiszek. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam ogromny zaszczyt zaprezentować niezwykłą kandydatkę na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. Pani mecenas Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, którą bardzo serdecznie witam [[Oklaski]] na galerii sejmowej, jest nie tylko bezpartyjną kandydatką rekomendowaną przez klub Lewicy, ale jest przede wszystkim kandydatką obywatelską, i to określenie w pełni odzwierciedla dzisiejszą sytuację. Popiera ją ponad 1100 organizacji społecznych, od lewa do prawa, od liberalnych po konserwatywne. Mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy takiej mobilizacji suwerena. Tak, suwerena. 1100 organizacji powiedziało, jak widzi funkcjonowanie tego urzędu. Nigdy wcześniej obywatele tak masowo nie połączyli się we wspólnych wysiłkach na rzecz powołania rzecznika. Wspólnota, współpraca, odwaga - to jest jej wizja funkcjonowania tego ustrojowego organu, jakim jest rzecznik praw obywatelskich. Kandydatka spotkała się z każdym klubem parlamentarnym i kołem. Każdy miał okazję zapoznać się z jej programem i pomysłem na pracę urzędu. Ten urząd nie jest ani nasz, ani wasz. Ten urząd należy do obywateli i obywatelek. Do rzecznika praw obywatelskich rocznie wpływa ponad 50 tys. skarg i próśb o wsparcie. To oznacza, że wypracowane do tej pory standardy pracy tego organu cieszą się niezwykłym społecznym zaufaniem. Nie zmarnujmy tego dorobku. Nie zmarnujmy tego potencjału, który od 30 lat realizuje urząd rzecznika praw obywatelskich. Każdy rzecznik na przestrzeni ostatnich trzech dekad naznaczył ten urząd swoją wizją, od pani prof. Łętowskiej po pana prof. Bodnara. Wierzę, że przedstawiana przeze mnie kandydatka dołoży swoją jakże cenną cegiełkę do funkcjonowania tego ustrojowego i niezwykle istotnego urzędu, jakim jest urząd rzecznika praw obywatelskich. Wysoka Izbo! Czas na zgodę.

I jest dobra okazja, żebyśmy ponadpolitycznie, ponadpartyjnie i poza sporem politycznym wybrali kogoś, kto będzie łączył, a przede wszystkim kogoś, kto będzie dbał o interes suwerena. Nie ma lepszego testu dla tego hasła i nowej jakości w polityce niż dzisiejsze głosowanie. Dorobek pani mec. Rudzińskiej-Bluszcz to przede wszystkim walka o człowieka i o jego sprawy. To będzie rzeczniczka ludzkich spraw. Czas na zgodę panie i panowie z Prawa i Sprawiedliwości. Czas na obywatelską rzeczniczkę. Dziękuję. W imieniu grupy posłów z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska kandydaturę przedstawi pan poseł Robert Kropiwnicki. Wysoka Izbo! Otóż mam niezmierny zaszczyt przedstawić kandydatkę na funkcję rzecznika praw obywatelskich, i to jest kluczowe, rzecznika praw obywatelskich, nie rzecznika praw polityków, nie kolejny łup polityczny, nie kolejne stanowisko dla przyjaciół, ale rzecznika praw obywatelskich. Kluczowe jest to, że to jest urząd, który ma chronić obywateli właśnie przed władzą, przed każdą władzą, zarówno przed tą najmniejszą - gminną, jak i przed wielkim ministrem, wielkim wicepremierem, premierem czy prezydentem.

O to chodzi w funkcji rzecznika.

Wszyscy będą wiedzieli, że chodzi o kolejny łup polityczny.

W starożytnym Rzymie przez prawie 500 lat funkcjonowała instytucja trybuna ludowego.

Lud przez 500 lat wybierał swoich przedstawicieli. Wiecie, kto zlikwidował trybunów? Powiedział wtedy, że to on będzie reprezentował lud. Wszyscy wiedzą, że jesteście po to, żeby sprawować władzę i to najczęściej we własnym interesie, a nie w interesie ludu.

Rzecznik polityków nie jest nikomu potrzebny, wszyscy potrzebują rzecznika dla ludzi, rzecznika praw obywatelskich.

Nie bójcie się tego wyboru. Pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz ma ogromne doświadczenie.

Jest duża szansa, że będzie miała poparcie Senatu.

Dlatego proszę was o poparcie pani Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, która będzie naprawdę dobrym rzecznikiem. Proszę teraz pana posła Jana Kanthaka o przedstawienie opinii komisji.

Panie Marszałku! W imieniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka przedstawiam opinię komisji dotyczącą wniosku o powołanie na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich pani Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. Odbyła się dyskusja. Po dyskusji odbyło się głosowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska.

Wysoka Izbo!

Jaki będzie wynik testu?

Wybieramy dziś rzecznika praw obywatelskich, rzecznika społeczeństwa.

Rzecznik nie musi podobać się władzy. Nie słyszałem żadnej merytorycznej uwagi do kandydatki. W kuluarach mówicie, że to świetna kandydatka. Nie odrzucajcie tej propozycji tylko dlatego, że nie macie własnej. To nie jest czas na targi polityczne i polityczne łupy. To nie jest czas na wystawianie partyjnych weksli, by uzyskać wysoką pozycję ustrojową. Ludzie są zagubieni, nie czują się bezpiecznie, nie są w stanie nadążyć za co chwilę zmieniającymi się decyzjami. Chcą rzecznika, do którego mogą się zwrócić w każdej sprawie. Interesów osób starszych, niesamodzielnych, z niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności nie można przecież nazwać prawicowymi lub lewicowymi. Rzecznik nie jest od przytakiwania decyzjom władzy, ani tej samorządowej, ani rządowej. Polki i Polacy mają prawo do rzecznika swoich praw. Pan premier Morawiecki wczoraj powiedział, że najważniejszą szczepionką na koronawirusa jest solidarność. Słowo „współpraca” odmieniał przez wszystkie przypadki. Dzisiaj jest okazja, żeby pan premier i jego obóz potwierdzili te słowa i udowodnili, że to nie są puste hasła. Dziś przeprowadzamy test na wiarygodność tych słów. To jest to miejsce, to jest ten czas. Wysoka Izbo! 9622, 10040, 12107 - codziennie nowa liczba dnia. To nie jest abstrakcyjna liczba, to liczba osób z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19. To liczby, za którymi stoją ludzkie tragedie, strach, ból. To godziny czekania na pobranie wymazu, przyjęcie na oddział. To kolejki karetek na podjazdach szpitali. To samotna choroba, czasami samotna śmierć. W tych ciężkich czasach musimy dostrzec, jak ważną funkcję pełni rzecznik praw obywatelskich. Rzecznik nie jest i nie może być posłusznym wykonawcą partyjnych zachcianek. To konstytucyjny urząd powołany do życia dla i przez obywateli. Czy wiedzą państwo, co łączy stowarzyszenie pomagające osobom uzależnionym od alkoholu w Andrychowie, Bydgoski Alarm Smogowy, warszawskie ZHP, fundację seniorów z Zielonej Góry czy Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica? Zapewne łączy ich to, że głosowali na wszystkich państwa tutaj, po każdej stronie tej Izby, ale przede wszystkim łączy ich przekonanie, że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich nie powinno być przedmiotem politycznych targów. Łączy ich zaufanie do koncepcji stojących za wyborem rzecznika ponad partyjnymi podziałami. Tych organizacji jest ponad 1100 i stoi za nimi ponad 1 mln Polek i Polaków. I wszyscy ci, którzy dzisiaj podniosą rękę przeciwko kandydatce na urząd rzecznika praw obywatelskich. Ojej... ...pokażą słynny palec Lichockiej wszystkim tym organizacjom. Ooo... ...i całemu społeczeństwu, które tę kandydaturę popiera. Pokażcie więc, wyciągnijcie rękę w stronę społeczeństwa w tym czarnym dniu [[Dzwonek]] dla praw kobiet, dla praw człowieka. Bardzo proszę. 2 minuty, panie pośle. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Zacznę od zwrócenia się do tej części sali sejmowej z pytaniem: Czy nie szkoda państwu tego wspaniałego dorobku instytucji, jaką jest urząd rzecznika praw obywatelskich, dorobku, który również śp. Janusz Kochanowski związany z waszym środowiskiem politycznym jako rzecznik praw obywatelskich tworzył?

Byliśmy jako kraj podziwiani za wspaniały wkład właśnie w budowanie tych niezwykłych instytucji w innych krajach. Dzisiaj, wprowadzając swoistego rodzaju paraliż, przekreślacie to państwo. A więc pytamy przy tej okazji: Czy nie szkoda tego dorobku, który tworzyli ludzie różnych poglądów, różnych opcji politycznych? Przejdę teraz do osoby pani mecenas Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. Co, szanowni państwo, jest złego w podkreślaniu równego dostępu do edukacji, równego dostępu do opieki zdrowotnej, we wskazywaniu obszarów ubóstwa, które - wśród najmłodszych niestety - są ciągle w naszym kraju obecne? Cóż złego jest we wskazywaniu wykluczenia cyfrowego, które dotyka sporą część naszego kraju? Czy to są kontrowersyjne obszary? Czy to są sprawy, które wypada nam dzisiaj negować w tej Izbie? I wreszcie bardzo duże i mocne poparcie obywatelskie przekonuje nas do tego, żeby z pełną odpowiedzialnością, jako Koalicja Polska, poprzeć osobę pani mecenas [[Dzwonek]] Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. Pan poseł Robert Winnicki, koło Konfederacji.

Wysoka Izbo! Art. 38 konstytucji mówi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

Warto w tym momencie podziękować sędziom Trybunału Konstytucyjnego za to, że takie orzeczenie wydali. Szanowni Państwo! Tak, konstytucja, konstytucja, konstytucja. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

Nie wstyd panu? To niech pan usiądzie i nie podnosi głosu wtedy, jak nie ma pan głosu. Ja tu słyszałem różne haniebne głosy i nie było takich awantur. Najwyższy czas, panie marszałku, Wysoka Izbo, żeby parlament Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno Sejm, jak i Senat, wybrał takiego rzecznika praw obywatelskich, który będzie gwarantował poszanowanie wszystkich praw obywatelskich, a zwłaszcza tego fundamentalnego, tego najważniejszego, czyli prawa do życia. Z całym szacunkiem dla pani mecenas: podczas prac komisji, podczas tych przesłuchań, jednoznacznej deklaracji w tej sprawie nie usłyszeliśmy. W związku z tym takiego poparcia udzielić nie możemy. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję.

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za powołaniem pani Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko rzecznika praw obywatelskich, zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm nie powołał pani Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. W związku z tym, że Sejm nie powołał rzecznika praw obywatelskich, procedura zostanie przeprowadzona ponownie.

Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny 19. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Czy ktoś z pań i panów posłów jeszcze chce się dopisać? Zamykam listę zgłoszonych. Bardzo proszę, pani

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tak zwany Trybunał Konstytucyjny tzw. wyrokiem sponiewierał polskie kobiety, pohańbił je, odebrał im godność i prawa człowieka, odebrał im ludzką podmiotowość, pozbawił je prawa do decydowania o sobie, o swoim życiu, zdrowiu i prawie do posiadania szczęśliwej rodziny. Polskie państwo rękami kadłubkowego Trybunału Konstytucyjnego zdradziło połowę swoich obywateli. Polski parlament nie może pozostać niemy i bierny wobec tej niegodziwości. Zgłaszam wniosek formalny o przerwę i zwołanie natychmiastowej debaty parlamentarnej, póki jeszcze nie założono kobietom knebla, póki jeszcze nie założono łańcuchów, póki jeszcze Straż Marszałkowska nie wynosi posłanek z sali parlamentarnej. Musimy rozpocząć debatę o liberalizacji ustawy aborcyjnej, o przywróceniu Polkom należnych im praw człowieka. Dziękuję bardzo.

Nie ma. Czy jest na sali pan poseł Tomasz Olichwer, Koalicja Obywatelska? Bardzo proszę, panie pośle.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Premierze! Zwracam się w tym miejscu do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, pracy i technologii pana Jarosława Gowina.

Tzw. zielona energia jest oczywiście z jednej strony jednym ze sposobów na zażegnanie kryzysu klimatycznego, który niszczy naszą planetę, lecz z drugiej strony uchwalana ustawa w sposób znaczny ograniczyła możliwość budownictwa mieszkalnego na terenie gmin, które przed wejściem w życie ustawy zdecydowały się na wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a wcześniej - do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, terenów pod budowę farmy wiatrowej.

Przykładem takiego stanu rzeczy jest jedna z gmin mojego okręgu wyborczego. W Wielowsi w powiecie gliwickim na długo przed wejściem w życie tzw. ustawy odległościowej samorząd gminny zdecydował się dać zielone światło budowie właśnie farmy wiatrowej. W 2016 r. Sejm, nie wsłuchawszy się w głos mieszkańców terenów, których ustawa dotyczy, postawił władze gmin w sytuacji bez wyjścia. Gminy stanęły przed wizją całkowitej blokady terenów pod budynki mieszkaniowe po upływie terminu obowiązywania przepisów przejściowych. W ostatnim czasie w mediach pojawiły się doniesienia, jakoby rząd Zjednoczonej Prawicy próbował naprawić popełniony w 2016 r. błąd i planował systemowe zmiany w zakresie farm wiatrowych w Polsce w postaci przedstawienia Sejmowi projektu ustawy w sprawie zmiany ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Z uwagi na powyższe zwracam się do pana premiera z prośbą o odpowiedź na następujące pytania: Czy ministerstwo planuje przedstawić Radzie Ministrów jakikolwiek projekt ustawy w sprawie zmiany ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych? Czy ministerstwo od 2016 r. otrzymało jakiekolwiek prośby o zmianę przepisów tej ustawy? Jakie zmiany ministerstwo planuje przedstawić w projekcie ustawy zapowiadanym jeszcze przez panią minister Jadwigę Emilewicz? Czy ministerstwo prowadziło jakiekolwiek konsultacje z władzami samorządowymi gmin, na których terenie powstają bądź istnieją elektrownie wiatrowe? I ostatnie: Dlaczego ministerstwo nie reagowało, nie wnioskowało do Sejmu o nieprzyjmowanie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych w 2016 r., skoro nie trudno było przewidzieć, że projekt ustawy praktycznie pozbawi gminy, na których terenie mieszczą się lub mieścić się będą elektrownie wiatrowe, terenów pod budownictwo mieszkaniowe? Proszę o wygłoszenie oświadczenia pana posła Władysława Teofila Bartoszewskiego, Koalicja Polska. Wysoka Izbo! To jest bardzo ważna funkcja konstytucyjna, rolą rzecznika jest głównie bycie adwokatem suwerena, czyli narodu, przeciwko wszystkim możliwym naruszeniom władzy i prawa poprzez organa administracji gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i centralnej oraz wszystkich urzędów państwowych, jak również ewentualnych złych działań polityków. Jest to wyjątkowo ważna funkcja.

W związku z tym organizacje społeczne w liczbie powyżej 1000 poparły kandydaturę pani Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. Dzisiaj głosami Prawa i Sprawiedliwości pani kandydatka Rudzińska-Bluszcz została odrzucona. Znaczy to, że PiS ma za nic organizacje społeczne i ich członków, a jednocześnie nie wypełnia swoich obowiązków politycznych, ponieważ żadnego innego kandydata nie zasugerował. Otóż jest postulatem Koalicji Polskiej, żeby rzecznik praw obywatelskich był wybierany w wyborach powszechnych przez samego suwerena. Ale chciałbym zaapelować do. O, widzę pana marszałka seniora. Panie marszałku, chciałbym zaapelować do pana jako seniora, przedstawiciela obozu władzy, żeby działać w tej mierze w zakresie takim, o jakim mówił wczoraj pan premier Morawiecki, czyli pewnego konsensusu. Tak się składa, że ja dobrze znałem śp. pana Janusza Kochanowskiego, byłego rzecznika praw obywatelskich, który zginął tragicznie, i pan Janusz Kochanowski był świetnym prawnikiem, ale się władzy nie kłaniał. Z tego powodu był nagrodzony nie tylko przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy tzw. znakiem jakości orkiestry, ale również dostał medal św. brata Alberta, dlatego że się zajmował niepełnosprawnymi, ubogimi i popierał organizacje pozarządowe. Chciałbym widzieć rzecznika, który działał niezależnie od swoich poglądów politycznych, a pan Kochanowski miał poglądy konserwatywne, ale wiedział, że jego funkcją jest kontrola władzy, a nie jej schlebianie. Ja bym bardzo prosił, składam prośbę na ręce pana marszałka seniora, żeby pan marszałek zaapelował do swojego obozu politycznego, żebyśmy wybrali osobę kompetentną, [[Dzwonek]] właściwą, moralną i prawą. Cieszę się, że pan marszałek senior przyjął z uwagą stanowisko Koalicji Polskiej, które mówi, że rzecznika praw obywatelskich należy wybierać w wyborach powszechnych.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wysłuchałem z wielką uwagą stanowiska przedstawionego przez pana Bartoszewskiego w imieniu PSL-u, Koalicji Polskiej, formacji Kukiz i oczywiście z bardzo wieloma uwagami się zgadzam. Szczególnie z tymi, które wskazują na konieczność konsensusu w sprawie kontroli władzy. Ponieważ została przywołana osoba śp. pana Kochanowskiego, który poległ nad Smoleńskiem, apeluję do Koalicji Polskiej, do wszystkich posłów, by poparli działania komisji badającej dramat smoleński i by razem wystąpili w sprawie kontroli ówczesnej władzy - pana premiera Donalda Tuska - która oddała całe postępowanie w ręce rosyjskie, co sprawia olbrzymie kłopoty i trudności w badaniu tego dramatu, który - nie ma wątpliwości - nastąpił na skutek eksplozji, na skutek zamachu, którego dokonano. Bardzo dziękuję panu Bartoszewskiemu za przywołanie obowiązku, jaki spada na tę Izbę, by wspólnie w ramach konsensusu kontrolować władzę, by nie kłamać i by w sprawach najważniejszych dla Polski być razem. Jestem przekonany, że tak właśnie będzie we wszystkich tych ważnych sprawach. Proszę teraz o wygłoszenie oświadczenia pana posła Tadeusza Tomaszewskiego, Lewica. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W ostatnich dniach poza informacjami dotyczącymi ilości zakażeń na COVID-19 dostajemy też dramatyczne listy od obywateli w kontekście nowego projektu listy refundacji leków, który ma obowiązywać od 1 listopada 2020 r. Pani Lidia pisze: Rok 2020 nazywany jest rokiem raka płuc. Nigdy nie przypuszczałam, że kiedykolwiek będzie dla mnie rokiem raka płuc, początkiem mojego życia z rakiem płuc. Jestem młodą osobą, nigdy nie paliłam papierosów. Diagnoza, którą usłyszałam od lekarzy po operacji, była okrutna: Ma pani złośliwego raka płuc. Jako pacjentka z rakiem płuc chcę być leczona zgodnie ze standardami leczenia w innych państwach europejskich - lekami innowacyjnymi i skutecznymi. Ogłoszony właśnie nowy projekt refundacji leków, który ma obowiązywać od 1 listopada br., pomija w nim innowacyjne terapie. Dlatego w imieniu środowiska pacjentów z rakiem płuc i ich rodzin pragnę wyrazić swoje głębokie rozczarowanie ponownym nieumieszczeniem na tej liście refundowanych leków innowacyjnej terapii niedrobnokomórkowego raka płuc u osób z ekspresją PD-L1 poniżej 50. Oznacza to, że nadal znacząca grupa chorych wciąż pozbawiona będzie dostępu do przełomowej opcji leczenia, rekomendowanej i dostępnej w 25 krajach europejskich, m.in. w Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze czy Rumunii. W Polsce każdego dnia z powodu raka płuc umierają 63 osoby - wczoraj 63, dzisiaj 63, jutro 63. One nie mają czasu czekać na kolejne listy refundacyjne. Wydłużenie i poprawienie jakości życia tych chorych jest w pełni uzależnione od dostępu do bezpiecznych leków o udowodnionej skuteczności. Niestety brak dostępu do tego leku na liście refundowanej w dalszym ciągu im tę szansę odbiera.

Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani marszałek. Przejęty przez Prawo i Sprawiedliwość Trybunał Konstytucyjny na jego rozkaz wprowadził całkowity zakaz przerywania ciąży, tym samym zniewalając Polki i zmuszając je do rodzenia dzieci nawet wtedy, kiedy one umrą, dzieci bez twarzy, dzieci bez mózgu. Będą zmuszone, co jest największą torturą, obserwować cierpienia tych dzieci. Tym samym Trybunał Konstytucyjny zrównał Polskę Dudy i Kaczyńskiego z reżimami totalitarnymi, gdzie również obowiązywał całkowity zakaz aborcji, a więc z III Rzeszą Hitlera, ze Związkiem Radzieckim Stalina i wreszcie z reżimem Ceaucescu w Rumunii. Nie ma na to zgody Lewicy, tym bardziej że ten wniosek jest najbardziej skandaliczny, dlatego że sam Trybunał Konstytucyjny, który powinien stać na straży praw konstytucyjnych kobiet, właśnie prawa konstytucyjne kobiet łamie. A wiec prawo kobiet do godności. Nikt bowiem nie zaprzeczy, że kobieta zmuszona do rodzenia w mękach dziecka z wadami jest pozbawiona godności, jej godność została złamana. Jeżeli nie mogą o sobie decydować, ich wolność legła w gruzach. Wreszcie konstytucja gwarantuje wszystkim, w tym również Polkom, życie wolne od tortury. Przecież to, z czym będą miały teraz do czynienia, to jest największa tortura, jaką można sobie wyobrazić. Ale Lewica nigdy nie zaprzestanie walczyć o prawa kobiet. My do końca, aż do skutku, będziemy o te prawa walczyć i już dzisiaj zapowiadam, że złożymy do Trybunału Konstytucyjnego wniosek, który wykaże, że konstytucja i konstytucyjne prawa kobiet są w Polsce łamane i są łamane przez Trybunał Konstytucyjny. Prędzej czy później - mam nadzieję, prędzej - Polki odzyskają swoje prawa do decydowania, do godności, do życia w wolnym kraju, do życia w kraju europejskim. My nie możemy być zniewolone, pozbawione swoich praw. Dziękuję bardzo. Proszę teraz o wygłoszenie oświadczenia pana posła Waldemara Andzela, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski jest zdobycie moskiewskiego Kremla przez polską armię z hetmanem Stanisławem Żółkiewskim na czele. Polacy byli pierwszymi Europejczykami, którzy zdobyli stolicę Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Wszystko zaczęło się od wojny polsko-rosyjskiej, która wybuchła w 1609 r. Rok później Polacy pokonali wielokrotnie liczniejsze wojska szwedzko-rosyjskie w bitwie pod Kłuszynem, a 9 października 1610 r. nasza armia pod dowództwem hetmana Stanisława Żółkiewskiego zajęła Kreml. Warto dodać, że stosunek liczebny wojsk Polski w odniesieniu do wojsk szwedzko-rosyjskich wynosił odpowiednio 5 tys. husarii, 2 tys. żołnierzy pomocniczych przeciwko 35-tysięcznej armii wroga. W wyniku przegranej tron utracił car Wasyl Szujski.

Moskiewska mennica wybijała monety z wizerunkiem Władysława IV Wazy, Polacy zaś okupowali Moskwę przez ponad 2 lata, wytrącając z rąk Rosjan najważniejszą bodaj dla każdego państwa wartość - suwerenność. Polacy dokonali tego, czego później nie udało się żadnej innej armii. Wojna polsko-rosyjska wraz ze zdobyciem Kremla określana jest w Rosji mianem wielkiej smuty. Następstwem wspomnianych przeze mnie wydarzeń był hołd ruski złożony przez cara Wasyla Szujskiego oraz jego braci Zygmuntowi III Wazie na Zamku Królewskim w Warszawie. Jest to jednak wydarzenie zapomniane o olbrzymiej doniosłości historycznej. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję. Proszę teraz o wygłoszenie oświadczenia panią poseł Monikę Falej, Lewica. Jeszcze kilka dni temu w ostródzkim szpitalu było ok. 40 zakażonych koronawirusem. Dziś jest ich prawie 150 i zaczyna brakować miejsc. W Olsztynie zamknięto oddział chirurgii w szpitalu miejskim. W Nowym Mieście Lubawskim zamknięto odział położniczo-ginekologiczny z powodu zakażenia personelu wirusem. Do odwołania wstrzymane zostały przyjęcia pacjentek. W szpitalach powiatowych w Mrągowie i Węgorzewie zamknięto oddziały wewnętrzne. W Morągu z powodu koronawirusa w szpitalu powiatowym zamknięto oddział neurologii. Szpital miejski w Elblągu w trybie natychmiastowym w całości ma zostać przekształcony w szpital zakaźny z uwagi na wysoki wzrost zakażeń koronawirusem. Taką decyzję podjął Artur Chojecki - wojewoda warmińsko-mazurski. I tak mogłabym wyliczać kolejne szpitale w województwie warmińsko-mazurskim czy też w całej Polsce. Tylko co dalej? Co robiliście przez lata? Co robiliście? Ustaliliście tylko, że epidemii nie ma, to wiemy. Co zrobiliście, żeby przygotować Polskę i Polaków, i województwo warmińsko-mazurskie, do drugiej fali epidemii, o której wiedzieli przecież wszyscy, wy też? Mamy prawo wiedzieć, a wy macie obowiązek prawny i moralny wytłumaczyć się z tego, co zostało zrobione, a co nie. Powinniście przygotować Polskę do drugiej fali epidemii i do tego, żeby osoby, które mają planowane operacje, mogły je mieć dokonane, bo to jest kwestia ich życia i zdrowia. Ale wy nie jesteście przygotowani. Jak osoby chore, nie na koronawirusa, będą zaopiekowane medycznie? Dziękuję. Bardzo dziękuję, pani poseł. Czy można prosić pana prowadzącego program, żeby trochę ciszej komunikował się z widzami?

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W grudniu br., czyli za 2 miesiące, minie rok od pierwszego czytania w Wysokiej Izbie obywatelskiego projektu ustawy w sprawie powołania Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy. Niestety, pomimo dramatycznego braku lekarzy i pielęgniarek w Polsce ten ważny projekt nadal leży w sejmowej zamrażarce. Od wielu lat polski system opieki zdrowotnej dławi się brakiem lekarzy, pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych. Rok temu, czyli w czasie, gdy rząd wiedział już o epidemii, Naczelna Rada Lekarska alarmowała, że w naszym kraju brakuje 70 tys. lekarzy. Za mało było pediatrów, psychiatrów dziecięcych, hematologów, onkologów, a nawet lekarzy rodzinnych. Polska zajęła ostatnie miejsce w Europie pod względem liczby lekarzy na 1 tys. mieszkańców według statystyk Unii Europejskiej. Niestety, zamiast zwiększenia liczby uczelni medycznych w Polsce i zwiększenia poziomu kształcenia, reakcją polityków PiS-u na te dane było schowanie głowy w piasek i zaniechanie działań. To typowa polityka ciepłej wody w kranie. Dzisiaj te zaniedbania mają dramatyczny skutek. Głównym problemem walki z epidemią, jak się okazuje, nie są dzisiaj pieniądze, nie są maseczki, nawet nie są respiratory, ale jest nim czynnik ludzki, czyli specjaliści. Bez nich nie zadziała respirator, bez nich nie da się leczyć pacjenta, a nawet pobrać mu próbki do badań czy bezpiecznie dowieźć do szpitala. Dzisiaj rząd, zamiast korzystać z wiedzy i zaangażowania lekarzy kształconych w Polsce, szuka ich na ukraińskich i kazachskich stepach. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Polski system opieki zdrowotnej musi być przygotowany na czas pokoju i na czas kryzysu. Bez wzrostu liczby lekarzy i pielęgniarek wszelkie reformy i wszelkie prowizorki będą miały ten sam efekt, jak przysłowiowe przelewanie z pustego w próżne. Obywatelski projekt ustawy w sprawie utworzenia Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy ma na celu zwiększenie liczby kształconych lekarzy i innej kadry medycznej. Uniwersytet w Bydgoszczy nie będzie powstawał kosztem innych uczelni. Dążymy do tego, by w wojewódzkie kujawsko-pomorskim były dwa uniwersytety kształcące kadrę medyczną zamiast jednego - jeden w Toruniu na bazie UMK i szpitali w Toruniu oraz drugi w Bydgoszczy na bazie nowego uniwersytetu i szpitali w Bydgoszczy. Bazę uniwersytecką można poszerzyć o inne szpitale wojewódzkie, np. w Grudziądzu, Inowrocławiu i Żninie. Przy tej koncepcji ośrodki uniwersyteckie w Bydgoszczy i Toruniu niczego nie stracą, a wręcz zyskają, podobnie jak polscy pacjenci i cały system opieki zdrowotnej. W związku z powyższym zwracam się z prośbą do pani marszałek, która ustala tematykę i terminy prac Sejmu (Dzwonek), aby wyznaczyła jak najszybciej termin posiedzenia komisji celem rozpoczęcia prac nad ustawą. Dzisiaj jest czas nie tylko myślenia o kopaniu studni, gdy wszystko się pali, ale także czas myślenia o przyszłości. Kadra lekarska i pielęgniarska kształcona na polskich uczelniach to właśnie zabezpieczenie przyszłości. Dlatego apeluję i proszę o pilne wdrożenie prac legislacyjnych nad tym obywatelskim projektem ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi. Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie. Informacja o wpływie interpelacji, zapytań oraz odpowiedzi na nie dostępna jest w Systemie Informacyjnym Sejmu. Na tym kończymy 19. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w Sekretariacie Posiedzeń Sejmu.